Panie i Panowie Posłowie! Zgłaszam wniosek formalny o przerwę w celu wprowadzenia do porządku obrad uchwały o negocjacjach w sprawie unijnego budżetu. Dziś z Sejmu musi wyjść jasny sygnał zarówno do naszych unijnych partnerów, jak i, przede wszystkim, do Polek i Polaków. Panie Premierze Morawiecki! Panu się wydaje, albo pan udaje, że walczy pan z Brukselą. Ale prawda jest taka, że walczy pan z polskimi samorządami, walczy pan z polskimi przedsiębiorcami. a nawet walczy pan z polskimi studentami. Niestety dziś polityka europejska rządu wygląda tak, jak wczoraj premier Kaczyński na spotkaniu z premierem Orbanem - z maską na oczach. A my dziś z szeroko otwartymi oczami chcemy głośno wykrzyczeć: Nie dla weta, tak dla Unii Europejskiej! Pani poseł, przede wszystkim chciałam panią poinformować, że, po pierwsze, uchwałę w tej sprawie podejmowaliśmy, po drugie, ten wniosek, zgodnie z tym, co ustaliliśmy na posiedzeniach Konwentu Seniorów i Prezydium Sejmu, idzie do Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Chciała pani złożyć, tzn. złożyła pani wniosek o przerwę, w związku z tym przegłosujemy wniosek o przerwę. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Z wnioskiem formalnym pan poseł Dariusz Klimczak, Koalicja Polska. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Zgłaszam wniosek formalny o przerwę w celu uzupełnienia porządku obrad o informację premiera na temat. narodowej strategii szczepień przeciw COVID-19. Te kilkanaście kartek to jest narodowa strategia czy ulotka informacyjna? Żądamy uszczegółowienia tej informacji, tym bardziej że rząd wczoraj poinformował, że jesteśmy przygotowani tylko na 180 tys. szczepień tygodniowo, co oznacza, że wszystkich Polaków zaszczepimy dopiero za 4 lata. Trzeba dać możliwość szczepienia farmaceutom w aptekach, tym bardziej że jest to możliwe w wielu krajach Unii Europejskiej. Mało tego, żądamy, żeby każda osoba, która zdecyduje się na szczepienie przeciw COVID-19, była zwolniona z wszelkiego rodzaju restrykcji, obostrzeń, limitów, w tym z obowiązku noszenia maseczki. Mało tego, żądamy, aby wszystkie szczepienia w Polsce były bezpłatne. Wie to każdy rodzic, który decyduje się, żeby jego dziecko zostało zaszczepione przeciw pneumokokom, bakteriom i innym wirusom, co wynika z kalendarza szczepień, ile to kosztuje. Od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Żądamy, żeby wziąć się za prawdziwą strategię szczepień w Polsce.

Jeszcze kilka miesięcy temu na tej sali premier Morawiecki cieszył się z ambitnego budżetu Unii Europejskiej, z ogromnych środków przyznanych Polsce na Fundusz Odbudowy. Europa otrząsnęła się z marazmu, Polska miała dostać dziesiątki miliardów euro na rozwój. Dzisiaj nastroje są zupełnie inne, stery w kraju przejął Zbigniew Ziobro, Polska jest o krok od utraty potężnych pieniędzy, pojawiają się nieodpowiedzialne głosy o polexicie. Polska z pierwszego i Polska z drugiego scenariusza to są dwie różne Polski. Ta druga jest po prostu dużo biedniejsza. Dlatego chcemy usłyszeć od rządu uczciwie, na co zabraknie pieniędzy, z czego rząd chce zrezygnować. Czy porozumienie, które podpisaliście z górnikami, idzie do kosza? Czy rezygnujemy z doganiania Europy i godzimy się na rolę montowni Niemiec na zawsze? To jest wniosek nieregulaminowy.

Ostatni wniosek formalny, pan poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Ja proszę o przerwę, Konwent Seniorów, o odwagę i o poddanie wreszcie pod głosowanie przywrócenia do porządku obrad projektu rezolucji, który zgłosiła grupa posłów na poprzednim posiedzeniu, projektu uchwały odpowiadającego na rezolucję Parlamentu Europejskiego. Naprawdę, ile jeszcze potrzebujecie państwo upokorzeń, żeby pisnąć chociaż słowo sprzeciwu wobec tego, co tutaj się dzieje?

Teraz Parlament Europejski się rozzuchwalił i już nie tylko recenzuje pracę polskiego Sejmu, ale wyręcza Trybunał Konstytucyjny. No i gdzie ten trójpodział władzy - tutaj też pytam opozycję - za który tutaj bohaterowie walczyli, za który poległ i zmartwychwstał pan Diduszko? Co się z tym stało? Konwentu też nie zwołam, a te uchwały są w komisjach: w Komisji Spraw Zagranicznych i w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, panie pośle. Dziękuję bardzo.

Proszę pana posła Piotra Polaka o przedstawienie sprawozdania komisji.

W imieniu Komisji Finansów Publicznych mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Sejm na 21. posiedzeniu w dniu 18 listopada skierował powyższy projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu jego rozpatrzenia. Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2020 r. wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył załączony projekt ustawy. Otóż w tym projekcie ustawy są dokonywane zmiany w kilku ustawach.

Tak jak powiedziałem, konkludując, Komisja Finansów Publicznych wnosi, aby Sejm uchwalił załączony projekt ustawy. Dziękuję serdecznie. Witam państwa. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Zapraszam serdecznie pana posła Zdzisława Sipierę, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Proszę, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Prezentując stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, chciałem zwrócić uwagę na kilka aspektów projektowanych w tej ustawie zmian. Zmiany, które wprowadza ta ustawa nowelizująca ustawę o podatku akcyzowym oraz niektóre inne ustawy, są pozytywne. Zmierzają w kierunku ułatwienia, przyspieszenia i zmniejszenia kosztów operacyjnych projektowanych regulacji. Zmiany, które są proponowane w niniejszej ustawie, będą miały pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Zastąpienie papierowych dokumentów stosowanych przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy dokumentem w postaci elektronicznej, tzw. e-DD, spowoduje przyspieszenie zwolnienia zabezpieczenia akcyzowego składanego przez podmiot, które następuje po zakończeniu przemieszczenia wyrobów. Ten sposób pozwoli przedsiębiorcom na szybsze dokonanie kolejnego przemieszczenia bądź też wykorzystanie w inny sposób środków finansowych pochodzących ze zwolnionego zabezpieczenia akcyzowego.

Wprowadzenie ww. zmiany zmniejszy też koszty administracyjne po stronie przedsiębiorców, m.in. poprzez zniesienie obowiązku kwartalnego składania zestawień wystawionych papierowych dokumentów dostawy. Wprowadzenie możliwości podziału przemieszczenia na terytorium innego państwa członkowskiego w przypadku przemieszczeń wyrobów energetycznych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w systemie EMCS usprawni operacje przemieszczania w tym zakresie i będzie miało pozytywny wpływ na szybkość zakończenia przemieszczeń.

W merytorycznej komisji nie było żadnych głosów, które by się temu przeciwstawiały, nie było nawet głosowania.

Jednocześnie w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o to, żeby ww. ustawę z tymi poprawkami przyjąć. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Na początku warto wspomnieć o tym, że część zmian, które zostały zaproponowane w pierwotnej wersji projektu, musiała ulec zmianie m.in. ze względu na kolizję z przepisami zawartymi w ustawie o doręczeniach elektronicznych, nad którą procedowano w ostatnim czasie. Ponownie okazało się również, że rządowy projekt ustawy trafił do Sejmu z licznymi błędami legislacyjnymi, które na szczęście zostały zweryfikowane przez Biuro Legislacyjne.

Wątpliwości budzą stosunkowo szerokie uprawnienia urzędników w zakresie uznaniowego decydowania o kwestiach, które dotychczas były uregulowane dość konkretnie, ale nie w sposób idealny. Wprowadzenie jednego rejestru podmiotów akcyzowych prowadzonego przez wyznaczony organ - co stanie się centralną elektroniczną rejestracją podmiotów w podatku akcyzowym - w miejsce dotychczas istniejących lokalnych rejestrów prowadzonych przez właściwych w sprawach akcyzy naczelników urzędów skarbowych co do zasady należy uznać za słuszne. W związku z tym dobrze się stało, że te zmiany będą wchodziły w życie w najbliższym czasie. Debatując nad tym projektem ustawy, który dotyczy m.in. podatku akcyzowego, należy odnieść się do kwestii związanej z samochodami hybrydowymi. Zgodnie z tym, co pan minister mówił, wychodzimy naprzeciw i też sprawdzamy, czy pan minister dotrzyma słowa, bo mówił o tym, że jest skłonny, żeby to zwolnienie z akcyzy dla samochodów hybrydowych przedłużyć. Wnioskujemy i postulujemy, żeby to przedłużyć do 2023 r., dlatego że od 1 stycznia już właściwie ona nie będzie obowiązywała. Analizując poszczególne przepisy omawianego projektu, należy uznać, że częściowo odpowiada on potrzebom, które zgłaszane są przez przedsiębiorców. Pozostaje nam wierzyć - a jednocześnie też tego pilnować - że w ostatniej chwili nie wprowadzi się zmian, które w negatywny sposób uderzą w podatników. Według tego, co słyszeliśmy przed chwilą od posła reprezentującego klub PiS, tych zmian chyba nie będzie. Natomiast za każdym razem należy wyraźnie podkreślać, że w tak trudnych czasach, jakie obecnie nastały, wspieranie przedsiębiorców jest kluczowe. Dlatego, tworząc każdy kolejny akt prawny, zwłaszcza z zakresu prawa podatkowego, trzeba pamiętać, że to właśnie oni tworzą polską gospodarkę, oni płacą podatki i te podatki powinny być dla nich jak najniższe, szczególnie w tym najtrudniejszym okresie, tak żeby te środki, które mają, które wypracowują, były przeznaczane na rozwój przedsiębiorstw, na płace, które też są w tym trudnym okresie zmniejszane. Szanowny Panie Ministrze! Składam poprawkę do tej ustawy. Tak jak powiedziałem, ona dotyczy.

Tak że to jest nasza poprawka. Zakładam, że ministerstwo pozytywnie się do tego odniesie, na co liczę i na co liczą też ludzie, którym zależy na dobru polskiego środowiska. Tak że popieramy ten projekt ustawy na tym etapie. Proszę też Wysoką Izbę o poparcie tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo panu posłowi. Zapraszam panią posłankę Anitę Sowińską, klub parlamentarny Lewica. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu parlamentarnego Lewicy w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 720. Niniejszy projekt przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i ma na celu, po pierwsze, uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie dokumentu w postaci elektronicznej, tzw. e-DD, z użyciem systemu EMCS, po drugie, objęcie monitorowaniem w systemie dodatkowych podmiotów sprzedających wyroby węglowe zwolnione z akcyzy, objęcie przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy, a także objęcie przemieszczeń eksportowanych wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Celem tej ustawy jest również uregulowanie zasad monitorowania przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem, uregulowanie zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów przemieszczanych na podstawie dokumentu elektronicznego, wprowadzenie centralnej, elektronicznej rejestracji podmiotów akcyzowych, w tym objęcie obowiązkiem podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, i umożliwienie dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju. Co do zasady popieramy przepisy, które zmierzają do cyfryzacji i uproszczenia procedur. W dłuższej perspektywie czasu jest to korzystne z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem, obniżki kosztów całego systemu, a także ze względu na zmniejszenie obiegu dokumentów papierowych, co ma korzystny wpływ na środowisko. Należy również podkreślić, że proponowane rozwiązania powinny przyczynić się do lepszej kontroli nad przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy lub wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy, a to powinno oznaczać lepszą ściągalność podatków.

Przewiduje się tutaj rozszerzenie katalogu podmiotów podlegających elektronicznemu zgłoszeniu rejestracyjnemu o podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, np. urzędy gmin, szkoły, szpitale, przedszkola czy jednostki Policji. W naszej ocenie zapis ten jest zbyt daleko idący, nakładający dodatkowe, skomplikowane obowiązki na małych odbiorców gazu. Chciałabym zaznaczyć, że ewentualne korzyści z rozszerzenia katalogu podmiotów podlegających elektronicznemu zgłoszeniu rejestracyjnemu są co najmniej wątpliwe, ponieważ przewóz gazu płynnego do takich odbiorców i tak będzie ściśle monitorowany z użyciem dokumentu elektronicznego e-DD. Ta grupa odbiorców nie generuje też ryzyka w zakresie podatku akcyzowego, nie tylko ze względu na jej rozdrobnienie, ale również dlatego, że gaz płynny w odróżnieniu od innych paliw typu benzyny czy oleje napędowe jest paliwem wymagającym posiadania specyficznej infrastruktury związanej z jego napełnianiem, transportem czy odessaniem. Dlatego też w naszej ocenie obowiązek rejestracyjny nie jest w tym wypadku działaniem adekwatnym do istniejącego ryzyka. Ewentualnie w przypadku braku możliwości odstąpienia od obowiązku rejestracji można rozważyć wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym to podmiot wysyłający będzie uprawniony do dokonania obowiązku rejestracyjnego względem podmiotów zużywających nieprowadzących działalności gospodarczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Krzysztofa Paszyka, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Chciałbym w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści przedstawić nasze stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 720.

Natomiast od początku lutego 2022 r. jedyną opcją będzie wykorzystanie systemu EMCS i dokumentów elektronicznych. Jak wynika z regulacji przedłożonej w projekcie, Ministerstwo Finansów planuje wydłużyć o rok okres, w trakcie którego będzie można stosować również papierowe dokumenty dostawy - do 31 stycznia 2022 r. W projekcie przewiduje się też zmiany w zakresie dokonywania obrotu wyrobami węglowymi objętymi zwolnieniem od akcyzy. Jak wynika z proponowanych zmian, w zależności od tego, czy dany pośredniczący podmiot węglowy dokonał w poprzednim roku sprzedaży wyrobów węglowych w ilości mniejszej lub większej niż 30 mln kg, od lutego 2022 r. będzie on bezwzględnie zobowiązany do dokonywania dostaw wyrobów węglowych z wykorzystaniem dokumentu e-DD.

Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Artura Dziambora, Koło Poselskie Konfederacja. Wysoka Izbo!

Natomiast warto porozmawiać o samym podatku akcyzowym przy okazji tej dyskusji.

Chciałbym powiedzieć, że można by równie dobrze dopisać na przykład wszystkie samochody. W ramach gestu dobrej woli samego rządu w tym ciężkim czasie jesteśmy ze wszystkich stron zachęcani do tego, żeby być eko, czyli żeby zamiast samochodu wybierać transport publiczny albo jeździć na hulajnogach lub rowerach, albo wybierać spacer.

Równolegle rząd regularnie przypomina o kupnie i zachęca do kupowania nowych samochodów.

W związku z tym, że Polaków nie stać masowo na nowe samochody, rząd, rozumiejąc to, powinien ułatwiać życie Polakom poprzez odpodatkowywanie ich i zmniejszanie kosztów ich życia.

To taki gest dobrej woli, bo jak wiemy, rząd dostaje dosyć sporą sumę dzięki temu, że jesteśmy - niektórzy z nas - na tyle bezczelni, że mamy czelność kupować tańsze samochody za granicą niż szukać w Polsce na naszym często drogim rynku.

Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Do zadania pytania zgłosił się pan poseł Jan Szopiński z klubu parlamentarnego Lewica. Zapraszam. Panie Marszałku!

A zatem przedsiębiorcy mają możliwość stosowania nowych zasad przemieszczania przy alternatywnej możliwości stosowania dotychczasowej, papierowej dokumentacji.

Mam pytanie do rządu: Czy małe firmy, małe przedsiębiorstwa mogą liczyć w tej sprawie na rekompensaty ze strony rządu? Kwestia druga. Otóż rząd pracował nad tą ustawą prawie rok. Przedsiębiorstwa, firmy, instytucje wypowiedziały się w listopadzie ub.r. Natomiast (Dzwonek) minister do spraw Unii Europejskiej wypowiedział się dopiero 2 listopada i - powiedziałbym dość dyplomatycznie - nie jest to wypowiedź najbardziej pozytywna dla tej ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Mirosław Suchoń, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam krótkie pytanie, ono dotyczy systemu teleinformatycznego.

Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Czy pan poseł Michał Szczerba jest na sali? Jestem przyzwyczajony do tego, że jest zawsze i wszędzie.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Chciałbym, panie ministrze, prosić pana o to, aby pan odpowiedział, czy zechce pan poprzeć poprawkę, o której mówił pan poseł Jaros, dotyczącą aut hybrydowych, chodzi o przedłużenie zwolnienia z podatku akcyzowego dla tych aut. A skoro mówimy już o podatkach, to chciałbym przypomnieć panu ministrowi, że czas, w którym żyjemy, czas pogłębiającego się kryzysu jest takim momentem, w którym powinniśmy ludzi, obywateli naszego kraju z podatków zwalniać i obniżać opłaty.

Bo na razie uchwaliliście państwo ich ze 40 i tak naprawdę pieniądze, które przekazujecie obywatelom np. na program 500+, wyciągacie obywatelom z kieszeni. Pani poseł Małgorzata Pępek, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Procedowana ustawa zmienia stosowanie warunków formalnych skorzystania ze zwolnień z opodatkowania podatkiem akcyzowym określonych wyrobów.

Z tego przepisu (Dzwonek) wynika, że zwolnienia te mają charakter obligatoryjny. A zatem zapisy procedowanej ustawy mogą być sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy przepisy zostaną zmienione tak, aby nie kolidowały ze wspomnianą wyżej dyrektywą? Pan poseł Paweł Papke, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W Prawie celnym wprowadza się stosowanie systemu EMCS PL2 i elektronicznego dokumentu dostawy e-DD do przemieszczeń na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od tejże akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Oczywiście co do całego tego projektu ustawy mam kilka pytań.